Wznawiam posiedzenie. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję poseł Martę Kubiak, która prowadzić będzie protokół i listę mówców. Pani poseł sekretarz nie ma żadnych komunikatów. Proszę państwa, przystąpimy do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu Sejmu.

Stwierdzam kworum.

Bardzo proszę, panie pośle. Nie ma. To pan poseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Za chwilę przed nami bardzo ważne głosowanie, kolejna szansa dla państwa, żeby udowodnić, że ustawa, nad którą wspólnie procedowaliśmy i którą wspólnie poparliśmy, nie służy wam do tego, by ukryć te wszystkie nieprawidłowości, które zdarzyły się przez ostatnie lata.

Niektórzy wasi posłowie okazali się przyzwoici, bo Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji poparła poprawkę Senatu. Wy natomiast na siłę, z uporem maniaka próbujecie zagwarantować bezkarność swoim. Apeluję o elementarną przyzwoitość, o takie spojrzenie w lustro i odpowiedzenie sobie, czy jesteście na tyle uczciwi, że możecie obejść się bez tej poprawki.

Proszę bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kiedy pan poseł, pan przewodniczący wchodził na tę trybunę, myślałem, że pan zechce przeprosić. Chodzi o przeprosiny za głosowanie swoich kolegów w Parlamencie Europejskim za rezolucją, która uderza w Polskę.

Tak że serdeczne gratulacje.

Otóż chciałbym zwrócić uwagę na trzy sprawy. Nie jest prawdą to, co pan powiedział, że to ma zagwarantować jakąś bezkarność itd.

I to także trzeba, Wysoka Izbo, powiedzieć. A teraz sprawa najważniejsza. Po co tak naprawdę zostało to wprowadzone?

Wówczas państwo mówiliście, że to przecież są jakieś bajki. Ale tego samego dnia sąd w Wielkopolsce skazał - i to kogo?

Tak. I to jest sytuacja, w której to nie ten wójt ani ci wszyscy samorządowcy, którzy postąpili w ten sposób, powinni być dzisiaj karani. Was to oczywiście nie interesuje, bo was to nie będzie dotyczyć. Bo wasza praca to tutaj wyjść, wystąpić z taką oracją, później pójść do zaprzyjaźnionej telewizji i na koniec dnia wysłać tweeta.

Tak że, Wysoka Izbo, radziłbym i naprawdę apelowałbym o to, by nie powielać tutaj absurdalnych tez, tak byśmy tę ustawę mogli przyjąć w dużo lepszej atmosferze. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, druk nr 2084. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 2083 i 2084) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, druk nr 2083. Marszałek Sejmu skierowała w dniu 12 marca 2022 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 12 marca 2022 r. wnosi: z 60 poprawek zgłoszonych przez Senat 43 poprawki odrzucić, a 17 poprawek przyjąć.

Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. Kto jest za odrzuceniem 1. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki. Kto jest za odrzuceniem 5. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za odrzuceniem 7. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za odrzuceniem 8. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę Senatu przyjął. Kto jest za odrzuceniem 9. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm przyjął poprawkę Senatu. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za odrzuceniem 10. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm przyjął poprawkę Senatu. Kto jest za odrzuceniem 11. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm przyjął poprawkę Senatu. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z państwa jest za odrzuceniem 12. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z państwa jest za odrzuceniem 13. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za odrzuceniem 14. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za odrzuceniem 15. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę Senatu przyjął. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 16. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Kto jest za odrzuceniem 17. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki Senatu. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 20. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

się nie wstrzymał. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę Senatu przyjął. Kto jest za odrzuceniem 37. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Kto jest za odrzuceniem 38. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za odrzuceniem 40. poprawki? Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawki Senatu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za odrzuceniem 47. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę Senatu. Kto jest za odrzuceniem 48. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki Senatu. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest za odrzuceniem 55. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

13 - za, przeciw - 441, nikt się nie wstrzymał. Sejm poprawkę Senatu przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto jest za odrzuceniem 56. poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm przyjął poprawkę Senatu. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za odrzuceniem 58. poprawki? Kto jest przeciw?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 12 marca. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą.

Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do wygłoszenia oświadczenia? Bardzo proszę. Zamykam listę. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wtedy chciałam w tej sprawie zabrać głos, ale z oczywistego powodu nie mogłam tego zrobić. 24 lutego na zawsze zapamiętamy jako dzień hańby Rosji i wszczęcia przez nią bestialskiej agresji na Ukrainę. Temat, który chciałam podjąć, może być niestety coraz bardziej aktualny.

Według danych WHO to czwarta najpoważniejsza choroba na świecie i jedna z głównych przyczyn samobójstw. W Polsce na depresję leczy się prawie 8 tys. dzieci i młodzieży. Nie ma danych, ile osób się nie leczy. Trudno mi o tym mówić, bo do mnie też docierają informacje o takich faktach, i to od osób, które znam. Pandemia też się do tego przyczyniła, bo ok. 44% nastolatków ma objawy depresji. Wpływ COVID jest ogromny, ale to jedynie wierzchołek góry lodowej. Jeszcze przed pandemią zbyt wiele dzieci było obciążonych problemami psychicznymi, niestety lekceważonymi przez państwo.

Średnio jedynie 2% pieniędzy przeznaczonych na opiekę zdrowotną wykorzystywanych jest na rozwiązanie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. To się musi zmienić, bo obawiam się, że będzie coraz gorzej. Według UNICEF rocznie niemal 46 tys. nastolatków popełnia samobójstwo powodowane zaburzeniami psychicznymi. Stąd mój gorący apel do rządu, aby nie czekać, bo choroby psychiczne będą coraz trudniejsze do pokonania. Tylko jedno zdanie dodam. Już słyszymy też o tym, że to obciążenie dotyczy również dzieci przyjeżdżających do nas z Ukrainy, więc to jest wielkie zadanie do wykonania, bardzo trudne. Ale musimy to zrobić. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z tego miejsca chciałem się dzisiaj zwrócić w dwóch ważnych sprawach przede wszystkim do premiera rządu i przedstawicieli organów państwowych w terenie, jakimi są wojewodowie.

Bardzo bym prosił o interwencję pana premiera w tej sprawie i szczególne zwrócenie uwagi wojewodów na ten problem w poszczególnych województwach. Jednocześnie prosiłbym o wsparcie wojewodów, którym podlegają poszczególne dworce PKP, na których znajdują się uchodźcy z Ukrainy, żeby jeszcze bardziej zintensyfikowali swoje działania i wspierali wolontariuszki i wolontariuszy, którzy bezpośrednio pomagają uchodźcom z Ukrainy. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę z najwyższym szacunkiem odnieść się do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy i innych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego, którzy pospieszyli z pomocą dla obywateli Ukrainy zarówno przebywających obecnie w ich ojczyźnie, jak i też tych, którzy uciekając przed śmiercią, dotarli do regionu Kujaw i Pomorza. Akcja pomocowa w Bydgoszczy i okolicy jest zakrojona na ogromną skalę. Jutro, 13 marca, o godz. 13 królewskie miasto Bydgoszcz zaprasza wszystkich na Wyspę Młyńską i do Młynów Rothera na koncert charytatywny na rzecz Ukrainy pod hasłem: ˝Jesteśmy z Wami!˝, Bydgoszcz dla Ukrainy. Wszyscy wykonawcy na tym koncercie zagrają za darmo, organizatorzy za przygotowanie imprezy także nie biorą ani złotówki. Cele są dwa. Po pierwsze, jest to pomoc dla naszych ukraińskich przyjaciół, którzy uciekając przed wojną, trafili do Bydgoszczy. Uchodźcy podczas imprezy będą mogli skonsultować się z lekarzami, prawnikami czy przedstawicielami agencji pracy, którzy odpowiedzą na pytanie, gdzie się leczyć, do którego urzędu się udać, aby uzyskać finansowe wsparcie na zaspokojenie konkretnych potrzeb danej rodziny. Drugi cel to zbiórka pieniędzy na przyszłość ukraińskich rodzin, które z dnia na dzień stały się naszymi sąsiadami już nie z kraju obok, ale z pokoju obok. Z tego miejsca proszę o wsparcie zbiórki i obecność na koncercie. Wspólnie bydgoszczanie chcą stworzyć fundusz pomocowy dla ukraińskich rodzin. Podczas koncertu będzie można wpłacać pieniądze do puszki wolontariuszy. Na wyspie staną też punkty pomocy dla obywateli Ukrainy. Tuż obok będą wolontariusze gotowi zaopiekować się dziećmi. Na miejscu będą pracować lekarze i pielęgniarki gotowi udzielić porad medycznych, a także prawnicy i przedstawiciele urzędu oraz agencji pracy z ofertami zatrudnienia. Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Jesteśmy z wami. Szanowni Państwo! Bydgoszcz tym koncertem dziękuje wszystkim pięknie za otwieranie swoich serc. Bo teraz Rzeczypospolita Polska i Ukraina, dwa państwa, to samo serce. Polska i Ukraina teraz to jedna wielka rodzina. Kijów, Warszawa - wspólna sprawa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiejsze oświadczenie mam na temat polskiej polityki zagranicznej w kontekście wojny na Ukrainie. Są to bardzo trudne dni dla naszych ukraińskich sąsiadów, jak również dla nas i innych europejskich narodów. Odpierać rosyjską agresję można na wiele sposobów, jednak to, co możemy zrobić, to skuteczna polityka zagraniczna ukazująca prawdziwe oblicze Władymira Putina. Polska prowadzi potężną misję dyplomatyczną. Kraje zachodnie powoli zaczęły mówić naszym głosem, ale trzeba iść jeszcze dalej. Od samego początku to Polska stawiała na twarde sankcje wobec Rosji. Najdotkliwszą sankcją dla Kremla będzie uniezależnienie się od polityki energetycznej Rosji. Mam głęboką nadzieję, że Niemcy zmienią swoje zdanie w zakresie Nord Stream 1, Nord Stream 2, które przez lata zasilały rosyjski budżet i pozwoliły na dzisiejsze barbarzyńskie ataki militarne. To m.in. te pieniądze sprawiły, że rosyjscy żołnierze podbijają Ukrainę, dokonując ludobójstwa, gwałtów i aktów terroru. Dlatego tak ważne jest, by Europa mówiła jednym głosem. Dzisiaj Ukraina, jutro Litwa, a pojutrze Polska. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Fryderyk Kapinos, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. Pan poseł Sławomir Skwarek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Inicjatywę ustawodawczą, o czym warto pamiętać i przypominać, podjął prezydent Lech Kaczyński. 1 marca to data, którą zaproponował prezes IPN Janusz Kurtyka w nawiązaniu do wykonanego tego dnia wyroku kary śmierci w mokotowskim więzieniu - katowni na siedmiu członkach zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W walkach podziemia niepodległościowego z władzą komunistyczną zginęło ok. 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych w wyniku sfingowanych procesów, wielu zmarło w katowniach UB. Tak, historia o nich długo milczała, ponieważ ˝żyli prawem wilka˝ 10 lat temu grupa pasjonatów i działaczy społecznych zorganizowała Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziś Fundacja Wolność i Demokracja jest organizatorem największego w Polsce biegu pamięci. Oddają hołd niezłomnym organizatorzy, ale przede wszystkim tysiące biegaczy, których łączy wspólna idea - bieg ku pamięci.

Dęblin, Firlej, Jabłonna, Lublin, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Sobieszyn, Stanin czy Świderki to tylko niektóre miejscowości województwa lubelskiego, w których odbył się 10., jubileuszowy bieg. Jestem dumny, że mogłem wziąć w nim udział, wspólnie z młodzieżą klas mundurowych z zespołu szkół w Sobieszynie. W tej okolicy ukrywał się i walczył mjr Marian Bernaciak ˝Orlik˝ Dlatego bieg liczy symboliczne 1963 m. Ziemia łukowska to teren konspiracyjnej działalności Antoniego Dołęgi. Nigdy się nie ujawnił, nigdy się nie poddał, ukrywany i wspierany przez lokalną społeczność, w szczególności społeczność gminy Trzebieszów.

Jak Inka i wielu innych zachował się tak, jak trzeba. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! W moim oświadczeniu poselskim pragnę zwrócić uwagę na niezwykłą życzliwość, szlachetność i wrażliwość na los drugiego człowieka drzemiące w polskim narodzie, jakie ujawniły się w chwili napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i powstania w związku z tym faktem 1,5-milionowej fali uchodźców, która do nas dotarła. Sytuacja ta ukazała ogromne pokłady niezwykłej dobroci, zdolności do poświęceń oraz empatii polskiego społeczeństwa, a dowodem na to jest fakt, że poza instytucjami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi oraz licznymi organizacjami charytatywnymi niosącymi pomoc spontanicznie zaangażowało się w tę pomoc tak wielu mieszkańców naszego kraju. Polacy, dzieląc się dobrem materialnym, bezinteresownie otworzyli przed potrzebującymi drzwi swoich domów, zapewniając nie tylko schronienie, ale i godne życie. Poświęcają swój czas, energię i pracę, ofiarowując różnorodne, szerokie wsparcie, dzieląc się wiedzą i zwykłą ludzką życzliwością, co zauważył i docenił cały świat. Taka szlachetna postawa wielu Polaków zachęca do naśladowania, uczy młode pokolenie właściwych postaw, napawa dumą i skłania do refleksji. Myślę, że to wielki zaszczyt żyć, pracować i mieszkać wśród tak wspaniałych ludzi, jakimi bez wątpienia są nasi rodacy, których bez wahania możemy nazwać bohaterami tego trudnego czasu zasługującymi na wielki szacunek i uznanie. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Takie oto refleksje nasunęły mi się na myśl i postanowiłem się nimi z państwem podzielić. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Od ponad 2 tygodni mamy do czynienia z ogromną tragedią, jaka dotknęła naszych bezpośrednich sąsiadów. Od 17 dni trwa wojna na Ukrainie. Z tego miejsca deklaruję solidarność z narodem ukraińskim i przekazuję wyrazy wdzięczności dla osób dobrej woli. My, Polacy, stanęliśmy na wysokości zadania. Nie zawiedliśmy, ponieważ w momentach kryzysowych nigdy nie zawodzimy. Składam podziękowania tym wszystkim, którzy zaangażowali się w bezpośrednią pomoc, otworzyli swoje serca i domy, dzielili się i dzielą pomocą, która dziś jest tak bardzo potrzebna. Dziękuję samorządowcom, którzy stoją na pierwszej linii tego kryzysu, szczególnie samorządowcom z terenów przygranicznych: prezydentowi i wiceprezydentowi Przemyśla Wojciechowi Bakunowi i Bogusławowi Świeżemu oraz burmistrzowi Ustrzyk Dolnych Bartoszowi Romowiczowi. W momencie gdy rządowe zarządzanie kryzysowe w naszym kraju nie funkcjonuje, oni stoją na wysokości zadania, zadania trudnego, skomplikowanego, z którym doskonale sobie radzą. Dziękuję prezydentowi miasta Krosna Piotrowi Przytockiemu oraz samorządowcom z odległych gmin, którzy przekazali pomoc dla uchodźców, przede wszystkim wójtowi gminy Lipka Przemysławowi Kurdziece i burmistrzowi gminy Krajenka Stefanowi Kiteli. Rodzina samorządowców, przedsiębiorców, wolontariuszy, strażaków ochotniczych straży pożarnych i osób dobrej woli, które nie są obojętne na tę tragedię, jest ogromna. Zbyt duża, by móc wszystkich tutaj wymienić. Wymieniałabym do wieczora. I to nasze szczęście, bo dzięki tym osobom możemy mieć poczucie faktycznej pomocy udzielanej naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. Chylę przed państwem czoła i bardzo dziękuję za waszą wrażliwość. Od ponad 2 tygodni Europa zdaje egzamin z człowieczeństwa i jestem przekonana, że my, Polacy, zdajemy ten egzamin na najwyższym poziomie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Atak Rosji na Ukrainę jest kolejnym aktem agresji obecnych władz Rosji, którego celem jest odbudowa mocarstwowej pozycji tego państwa po upadku Związku Radzieckiego. Kilkanaście lat temu siły rosyjskie zaatakowały Gruzję. Rosja wspierała i wspiera separatystyczne siły w Donbasie. W tej sytuacji warto przytoczyć słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które wypowiedział w Gruzji w 2008 r. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może przyjść czas na mój kraj, na Polskę. Słowa te w skrócie opisują rosyjskie plany związane z odtworzeniem imperium. Plany te były, są i będą zrozumiałe oraz widoczne dla większości mieszkańców Europy Wschodniej, a już na pewno będą one budziły grozę wśród obywateli państw, które w przeszłości wchodziły w skład Związku Radzieckiego. Mam na myśli tutaj Litwę, Łotwę i Estonię, a także Mołdawię, która po opanowaniu Ukrainy może stać się celem kolejnego ataku Rosji. Niestety niewielu polityków w krajach Europy Zachodniej te plany widzi i rozumie. A nawet jeżeli te plany widzą, to cynicznie udają, że nie widzą, bo partykularny i krótkoterminowy interes polityków rządzących w tych państwach jest taki, aby handlować z Rosją. Skutek tego jest taki, że państwa te nie dość, że same są uzależnione od dostaw nośników energii z Rosji, to jeszcze próbują uzależnić od gazu z Rosji inne państwa Unii Europejskiej. Klinicznym przykładem takiej polityki są Niemcy. Przedsiębiorstwa z tego kraju w porozumieniu z rosyjskim Gazpromem wybudowały na dnie Bałtyku dwa rurociągi łączące Rosję i Niemcy. Niemcy zgodnie z tymi planami miały stać się pośrednikiem sprzedaży rosyjskiego gazu do innych państw Europy. A więc na tej współpracy miała zarabiać nie tylko Rosja, ale także Niemcy.

Polska, odejdą od węgla jako źródła energii. Niemcy próbowały także w ramach transformacji energetycznej doprowadzić do tego, że kraje Europy miałyby zrezygnować nie tylko z węgla, ale także z energii jądrowej. Walka ze zmianami klimatycznymi stała się więc pretekstem do tego, żeby Europa była zależna od rosyjskiego gazu, który byłby dostarczany do Europy za pośrednictwem Niemiec. Wielu polityków krajów Unii Europejskiej po zakończeniu pełnienia funkcji publicznych została zatrudniona przez rosyjski Gazprom, na przykład pan Gerhard Schröeder, były kanclerz Niemiec. Dzisiaj, w dobie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, plany Rosji oraz Niemiec są widoczne i tylko sowicie opłacani rublami politycy niektórych krajów Unii Europejskiej nie są w stanie dojrzeć tych zależności.

Albo Unia Europejska będzie niezależna od rosyjskiego gazu, albo Unia Europejska nie będzie niezależna w ogóle. Dziękuję bardzo. Proszę, pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Pani Marszałek!

To jest szokujące, bo ten wyrok wypycha nas z Unii. Widzicie, tylko wyciągacie z tego zupełnie inne wnioski. Dla was to oznacza przyzwolenie na wyprowadzenie nas z systemu prawnego Unii. Kto wam dał do tego prawo? Ile procent Polek i Polaków jest za wyjściem Polski z Unii? Wczoraj ten Sejm przyjął ustawę o obronie Ojczyzny, ale nie pomoże nawet najlepsze uzbrojenie, jeśli zostaniemy sami. A do tego doprowadzacie, drukując w tym pseudosądzie orzeczenia godzące w system prawny Unii Europejskiej. Panie Wicepremierze ds. Bezpieczeństwa Kaczyński! Czy pan w ogóle czuje konsekwencje stwierdzenia: w Polsce prawa człowieka są niezgodne z polską konstytucją? Tym się pan zajmował w ukryciu przez ostatnie kilkanaście dni?

Pani poseł, Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo! Te rzesze osób zostały zaopatrzone, przenocowane, przewiezione w bezpieczne miejsca, nakarmione. To dzięki służbom pani wojewody Ewy Leniart, samorządu województwa podkarpackiego, samorządów powiatu lubaczowskiego, jeżeli chodzi o przejście w Budomierzu. Chciałabym się bardziej skupić na przejściu w Budomierzu, ale wiem, że na wszystkich przejściach, na całej granicy uchodźcy są tak samo traktowani.

Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy prowadzą punkt recepcyjny, którym zarządza w imieniu pani wojewody pan wójt gminy Wiesław Kapel, wraz z całą załogą, z wszystkimi jego pracownikami.

Bardzo dziękuję panu staroście Zenonowi Swatkowi, księdzu dziekanowi Andrzejowi Stopyrze, który przede wszystkim skupia się na pomocy w przygotowywaniu posiłków, ale też na przerzucaniu wszystkiego, co jest potrzebne, na drugą stronę, na Ukrainę. Bardzo serdecznie dziękuję Caritas Polska z jego dyrektorem Marcinem Iżyckim, rycerzom Kolumba, stowarzyszeniu miłośników Lwowa z panią prezes Marią Magoń, wszystkim wolontariuszom Szlachetnej Paczki z panią Danutą Kacprzak, ale też wszystkim harcerzom. Bardzo chciałabym w swoim imieniu przekazać wszystkim, których tu nie wymieniłam. Proszę was, obudźcie się wszyscy, zatrzymajcie tę straszną wojnę. Te dzieci, te matki z tymi dziećmi. Jestem, mówię tu w imieniu matek ukraińskich, dzieci ukraińskich: zatrzymajcie tę wojnę na Ukrainie. Nie dopuśćcie do tego, żeby ona rozkrwawiła całą Europę. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Włodzimierz Tomaszewski, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Szanowni Państwo Parlamentarzyści w Drodze! Ja już wielokrotnie podczas tej debaty sejmowej starałem się uzmysłowić, na czym polega zarządzanie kryzysowe. I ze zdumieniem stwierdzam, że duża część parlamentarzystów naprawdę nie rozumie, co to znaczy zarządzanie kryzysowe. W zarządzaniu kryzysowym dotyczącym sytuacji, kiedy jest zagrożenie stanem wojny, zagrożenie życia, bezpieczeństwa czy też zagrożenie epidemiczne, także to związane ze zdrowiem, działanie musi być szybkie. Każdy sektor w ramach tego zarządzania: i ten rządowy, i ten samorządowy, i różne podmioty publiczne, które są przewidziane w systemie tego zarządzania, musi działać z wyprzedzeniem. Działanie z wyprzedzeniem oznacza, że nie wszystkie elementy, które są określone w ustawach, w prawie, są przewidujące.

W związku z tym ze zdziwieniem przyjmuję fakt, że regulacje, które były przewidziane w ustawie, nad którą debatowaliśmy w zakresie dotyczącym pomocy obywatelom Ukrainy, ale chodzi o zasady obowiązujące w każdym stanie zagrożenia, nie zostały przyjęte. Dziwię się w ogóle, że funkcjonariusze publiczni, zwłaszcza ci, którzy krytykują np. działanie części sektora publicznego, nie rozumieją, że mają obowiązek podejmować decyzje: i finansowe, i materialne, ale im nie może nic grozić. Oni muszą mieć pewność, że ich działanie będzie przyjęte i że nie będą z tego tytułu sądzeni, skazywani, bo to byłoby absurdem.

Mam nadzieję, że nadrobimy to, co zostało dzisiaj czy we wcześniejszych debatach zakwestionowane z powodu braku zrozumienia, na czym polega zarządzanie kryzysowe. I to chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, bo walki polityczne nie ma mają tutaj żadnego znaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.